Marszałek Sejmu pani Elżbieta Witek zaprasza parlamentarzystów na pokaz świątecznego mappingu gmachu Sejmu przed wejściem głównym. Ponadto informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji: - do Spraw Petycji - godz. 10.30, - Etyki Poselskiej - godz. 10.30, - Polityki Senioralnej - godz. 13, - Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - godz. 13, - Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - godz. 13, - Spraw Zagranicznych - godz. 14, - Infrastruktury - godz. 14.30, - Finansów Publicznych - godz. 14.30, Zdrowia - godz. 15, - Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii - godz. 15, - Obrony Narodowej - godz. 16, - Finansów Publicznych - godz. 16, - Sprawiedliwości i Praw Człowieka - godz. 16.30, - Łączności z Polakami za Granicą - godz. 17.

Dziękuję panu posłowi. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość wycofał zgłoszoną informację bieżącą. W związku z tym punkt 17. porządku dziennego stał się bezprzedmiotowy. Grupa posłów przedłożyła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, druk nr 68. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący pierwsze czytanie tego projektu. Projekty to odpowiednio druki nr 63 i 62. W związku z tym, na podstawie art. 95b regulaminu Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące pierwsze czytania tych projektów ustaw. Rada Ministrów złożyła autopoprawkę do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, druk nr 45-A. W związku z tym, na podstawie art. 95b regulaminu Sejmu, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący pierwsze czytanie tego projektu ustawy wraz z autopoprawką. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, druk nr 93. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciw!

Za chwileczkę przystąpimy do głosowania. Wnioski formalne będą, proszę państwa.

Przystępujemy do głosowania. Będą wnioski formalne, proszę państwa. Pani poseł, będą wnioski formalne.

Kto z pań i panów. Kto z pań i panów posłów jest za wyrażeniem zgody na zastosowanie art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm propozycję odrzucił. Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, druk nr 69. Na posiedzeniu Konwentu Seniorów zgłoszono sprzeciw wobec propozycji uzupełnienia porządku dziennego o pierwsze czytanie tego projektu. Jest to, w myśl art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu, punkt sporny porządku dziennego. Propozycję uzupełnienia porządku dziennego o ten punkt poddam pod głosowanie. Przypominam, że zgodnie z art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu głosowanie to nie jest poprzedzone debatą ani zadawaniem pytań. Kto z pań i panów posłów jest za uzupełnieniem porządku dziennego o punkt w brzmieniu: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, druk nr 69, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zaraz sprawdzimy. Nie działa u pana? Proszę sprawdzić.

Sejm propozycję przyjął. Panie pośle, przepraszam, działa? Prezydium Sejmu proponuje, aby w dyskusjach nad dodanymi punktami porządku dziennego Sejm wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycje przyjął. W którym punkcie? Przy Sądzie Najwyższym?

Jest wniosek przeciwny. Pani Marszałek! Składam wniosek przeciwny. Pozostańmy przy 5 minutach. Proszę państwa, panie pośle, bardzo pana proszę. Tylko państwo zgłosiliście sprzeciw, a padł wniosek przeciwny. Jeżeli składamy wniosek, to chyba mamy prawo uzasadnić, skoro pan marszałek nawet nie wie, czemu się sprzeciwia. I chodzi o to, żeby również ci, którzy nas oglądają, wiedzieli, o czym rozmawiamy.

A my chcemy, żeby ta debata trwała dłużej niż 5 minut. A to głosowanie jest po to, żeby państwo, opinia publiczna, Polacy wiedzieli, że my chcemy prawdziwej debaty, a nie debaty 5-minutowej. Nie, panie pośle - nie „pani marszałek” Było posiedzenie Prezydium Sejmu, nie było sprzeciwu, Konwent Seniorów również był o tym poinformowany, więc bardzo proszę być precyzyjnym. Przystępujemy do głosowania nad propozycją Prezydium Sejmu. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem propozycji Prezydium Sejmu wysłuchania 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła w dyskusji nad tym punktem obrad, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm propozycję Prezydium przyjął.

Panie pośle, to jest nieprawda. Pani poseł, nie pierwszy raz głosujemy i mówimy o wnioskach formalnych, za każdym razem była 1 minuta. Mamy w tym momencie do czynienia z jednym z naprawdę najsilniejszych ataków na niezależność wymiaru sprawiedliwości. Ja wnoszę o przerwę i o to, aby zobowiązała pani Ministerstwo Sprawiedliwości do ujawnienia, czy ta ustawa represyjna nie została przygotowana po to, aby była projektem mającym zapewnić bezkarność politykom PiS-u - szereg afer, o których się dowiadujemy, od afery Banasia, przez ustawę o więziennictwie. Musimy to wiedzieć, bo jeżeli ta ustawa represyjna zostanie uchwalona, to sądy zamienią się po prostu w zabawki w rękach polityków PiS-u, a politycy PiS-u staną się bezkarną kastą wyjętą spod prawa. Ta ustawa wysadza w powietrze Oklaski) fundament niezależnego wymiaru sprawiedliwości, idzie w zupełnie odwrotnym kierunku niż orzecznictwo unijnego Trybunału, podważa podstawowe zasady, na jakich jest oparta Unia Europejska.

Kto z pań i panów posłów jest za ogłoszeniem przerwy, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że wniosek został odrzucony.

Wysoka Izbo! Składam wniosek formalny w myśl art. 184 ust. 1 i 3 pkt 1 o ogłoszenie godzinnej przerwy i zwołanie. Konwentu Seniorów celem przedstawienia właśnie Konwentowi, a potem całemu Sejmowi, uzasadnienia, dlaczego pani marszałek nie zastosowała art. 34 ust. 8 regulaminu, zgodnie z którym może skierować projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej celem wyrażenia opinii. Proszę nie krzyczeć i nie przeszkadzać. na względzie to, że zarówno opinie zewnętrzne, np. Sądu Najwyższego czy rzecznika praw obywatelskich, jak i, przede wszystkim, Biura Analiz Sejmowych mówią o tym, że są w tej ustawie zapisy, które naruszyć mogą zasadę niezawisłości sędziowskiej. Zacytuję: „Zapisy te rodzą poważne ryzyko stwierdzenia naruszenia zasady niezależności i bezstronności sędziowskiej” Dlaczego pani marszałek nie skierowała tej ustawy do Komisji Ustawodawczej, mimo że bardzo często, zwłaszcza co do projektów opozycyjnych, korzystano permanentnie z tego właśnie przepisu? Jak pani sama stwierdziła, marszałek może.

Bardzo proszę. 1 minuta, panie pośle. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Zwracam się z wnioskiem formalnym o przerwę i zwołanie posiedzenia Konwentu Seniorów celem uzupełnienia porządku obrad o informację prezesa Rady Ministrów o ostatnim szczycie Rady Unii Europejskiej. Po raz kolejny Polska ogłosiła sukces, nie wchodząc do rozstrzygnięć, które dotyczą 2050 r. i neutralności klimatycznej. Chciałbym, żeby Wysoka Izba została poinformowana, czy możemy w takim razie na tym etapie korzystać z Funduszu Solidarności w wysokości 100 mld zł, czy będziemy objęci tą pomocą, i jakie są wieloletnie ramy finansowe dotyczące właśnie polityki spójności i wspólnej polityki rolnej. Ponieważ premier ogłosił sukces - jako jedyny kraj nie przyjęliśmy tych zobowiązań - więc bardzo proszę panią marszałek o zwołanie Konwentu Seniorów i uzupełnienie dzisiejszego porządku obrad o tę informację.

Minuta, panie pośle.

Nie doszło do tego. Było posiedzenie dwunastego, a Komisja do Spraw Służb Specjalnych została zwołana na jutro na godz. 13, wtedy, kiedy są głosowania. Czyli mam prawo domniemywać, że pani z premedytacją nie doprowadziła do tego, żeby było posiedzenie Komisji do Spraw Służb Specjalnych w tej sprawie. Wasza determinacja w ukrywaniu tej sprawy pokazuje, jak duża jest tego skala. My mamy prawo domniemywać, że krakowscy sutenerzy nie tylko dzwonią do Banasia, ale może dzwonią jeszcze do Sasina. To jest wasza sprawa, wasza afera. Panie pośle, ja bardzo bym prosiła pana. Panie pośle, ja bardzo bym prosiła pana o to, żeby pan ważył słowa. Na posiedzeniu Konwentu Seniorów, kiedy o tym mówiliśmy, ja słuchałam tej konferencji prasowej, na posiedzeniu Konwentu i Prezydium, kiedy tę sprawę omawialiśmy, powiedziałam, że skierowałam wnioski - oba wnioski, bo były dwa - do Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Podałam przybliżoną datę, bo wtedy myślałam, że będzie to osiemnastego. Z pewnością ulegnie to zmianie, więc proszę nie wkładać w moje usta.

Nie ma potrzeby prostowania, dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana posła Sławomira Nitrasa, Koalicja Obywatelska. Również wniosek formalny. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Myślę, pani marszałek, że pani też nie jest zadowolona z przebiegu tych porannych... początku tych obrad. Ale dlatego, że my oczekujemy, że parlament będzie miejscem, gdzie będziemy realnie debatować. Pani marszałek, pani mówi, że będzie wyjaśnienie, ale przecież sprawa Banasia to są 2 tygodnie. 2 tygodnie i nie mamy wyjaśnienia. Pani marszałek poinformowała nas przed chwilą, że zwróciła się do premiera o to, kiedy premier będzie mógł do parlamentu przyjść, po to żeby przed parlamentem złożyć informację, co postanowił na szczycie. A na szczycie jako jedyny nie bierze udziału w ważnej polityce. Przed parlamentem. Nie uzyskał zgody parlamentu na taką decyzję i nie czuje się zobowiązany nawet do tego, żeby przyjść i parlament poinformować, dlaczego podjął taką decyzję na szczycie. Pani marszałek, my oczekujemy, że pani nie będzie tylko dla nas miła, tylko że pani sprawi, że parlament będzie sprawował realną kontrolę nad rządem. Chciałam panu powiedzieć, że ja. Nie, panie pośle, przede wszystkim muszę się zwrócić do premiera rządu, ponieważ znam kalendarz Sejmu, natomiast nie znam kalendarza pracy rządu i kalendarza pana premiera.

Ale jest też premierem. Panie pośle, nie było wniosku formalnego, w związku z tym nie będziemy głosować, bo nie mamy nad czym. Też wniosek formalny. W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 chciałbym się zwrócić w trybie art. 173 ust. 2 regulaminu o przerwę oraz zwołanie Konwentu Seniorów w celu. Bo my składamy prośbę o uzupełnienie porządku obrad właśnie o informację dotyczącą efektów ostatniej Rady Europejskiej, w tym dotyczącą neutralności klimatycznej do roku 2050, ale również celów średniookresowych do roku 2030, gdzie podnosi się, czy zamierza się podnieść, te cele średniookresowe do prawie 55% redukcji. I również na temat wieloletnich ram finansowych, bowiem to także było przedmiotem obrad, a to ma ogromny wpływ na wszystkie te cele, które są określone właśnie w kwestiach neutralności klimatycznej do roku 2050. Przed chwileczką to wyjaśniałam. Proszę pana posła Krzysztofa Śmiszka z Lewicy. Bardzo proszę, minuta, panie pośle. Wysoka Izbo! Mamy dzisiaj do czynienia z hucpą. Z hucpą nie tylko na poziomie legislacyjnym, ale też śmianiem się w twarz całemu społeczeństwu. Jak możemy jako posłowie w imieniu narodu pracować nad taką ustawą, skoro mamy kilka godzin na to, żeby się do tego przygotować? Szanowni państwo, w tym miejscu chciałbym też podziękować tym tysiącom ludzi, którzy wczoraj protestowali i dzisiaj protestują przed sądami. To dzięki wam czujemy tutaj siłę i będziemy dzisiaj walczyć o każdy przecinek w tej ustawie. Musimy porozmawiać poważnie o tym, jak wygląda program posiedzeń Sejmu, i zdjąć tę haniebną ustawę z porządku obrad. Panie pośle, chciałam tylko sprostować, ponieważ to nie jest tak, że wniosek, projekt wpłynął teraz. 7 dni wcześniej, zgodnie z regulaminem, wpłynął i wszyscy. Nie, nie, panie pośle. Tak że proszę być precyzyjnym. Porządku nie będziemy zmieniać, więc przerwy też nie będę ogłaszała, bo to jest też wniosek tożsamy. Proszę teraz pana posła Michała Szczerbę, Koalicja Obywatelska, także z wnioskiem formalnym. Bardzo proszę, panie pośle. Wysoka Izbo! Jeszcze ustawa kagańcowa, ustawa represyjna nie została uchwalona przez Sejm, a już mamy pismo prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego z 16 grudnia do prokuratorów regionalnych w sprawie wszczynania postępowań przeciwko sędziom, którzy stosują wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. pisze do prokuratorów, że każdorazowo, kiedy jest kwestionowany status sędziego, prokuratorzy muszą składać w tej sprawie wnioski do rzeczników dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych i rzecznika dyscyplinarnego sędziów Sądu Najwyższego. Szanowni Państwo!

Bardzo proszę.

Fakt, że rozpoczynacie państwo kolejną batalię z wymiarem sprawiedliwości, nie zwalnia was z obowiązku poinformowania opinii publicznej o tym, co dzieje się w Najwyższej Izbie Kontroli. Dziękuję, pani poseł.

Wysoki Sejmie! Proszę o przerwę, zwołanie Konwentu Seniorów i wprowadzenie do porządku obrad tematu, [[Wesołość na sali]] który dotyka tak naprawdę nas wszystkich.

Jeżeli te przepisy nie ulegną zmianie, to 1 stycznia tysiące firm, które zajmują się wywozem odpadów komunalnych z naszych domów, z naszych mieszkań, nie będą realizowały tych zadań. Bardzo proszę o wprowadzenie tego punktu do porządku obrad. Nie ogłoszę przerwy z tego samego powodu, który podałam przed chwilą. Proszę, jeszcze dwa wnioski formalne. Zwracam się w trybie art. 187 ust. 3 o zwołanie przerwy, w czasie której. Konwent Seniorów zmieni decyzję pani marszałek - czy też pani marszałek rozważy zmianę swojej decyzji - w sprawie ograniczenia ilości posłów i posłanek, którzy mogą zabrać głos w debacie o sądach powszechnych. Wczoraj w Polsce dziesiątki tysięcy Polek i Polaków zebrało się na ulicach ponad 200 miast. Tymczasem uniemożliwia się nam zabranie głosu. Ja oraz moje koleżanki i koledzy siedzący na sali nie możemy zapisać się do debaty i przekazać, co Polki i Polacy myślą na temat tej ustawy, ponieważ pani marszałek odebrała nam dzisiaj głos. To jest po prostu niedopuszczalne.

Nie pani marszałek, tylko Prezydium Sejmu podjęło taką decyzję. Konwent zaopiniował tę decyzję bez zastrzeżeń, w związku z tym proszę nie wprowadzać w błąd tych, którzy nas słuchają. To nie jest decyzja marszałka.

Prawda?

Bardzo proszę. Pani Marszałek! Na podstawie art. 184 zwracam się do pani z prośbą o zmianę sposobu prowadzenia obrad.

Dziękuję bardzo.

Konfederacja ma jedno pytanie, nie 11, panie pośle. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 18. porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 68) Proszę pana posła Marcina Porzucka o przedstawienie uzasadnienia projektu

Proszę państwa, żeby umożliwić panu posłowi wystąpienie, bardzo proszę o wyciszenie rozmów, ewentualnie o przeniesienie ich do kuluarów, a posłów zainteresowanych tym punktem porządku dziennego proszę o zajęcie miejsc. Bardzo proszę, panie pośle. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W ostatnich latach obserwujemy silne oddziaływanie trendów technologicznych i biznesowych na sektor energetyczny oraz motoryzacyjny. Nacisk na redukcję emisji gazów cieplarnianych, stałe ulepszanie technologii magazynowania energii czy rosnąca popularność i efektywność paliw alternatywnych powodują pojawianie się nowych rozwiązań. Rząd opracował szereg dokumentów wspierających rozwój elektromobilności i paliw alternatywnych w obszarze transportu. Zostały opracowane również narzędzia finansowania tych pozytywnych zmian. Jednym z nich jest powołany Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, którego celem jest wsparcie rozwoju elektromobilności, infrastruktury, paliw alternatywnych oraz rynku tych paliw. Istotnym elementem działań funduszu będzie udzielanie wsparcia dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców na zakup pojazdów elektrycznych. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wsparcie, jakie będzie udzielane ze środków funduszu, podlega opodatkowaniu, zarówno w przypadku osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Obecnie funkcjonujące wyłączenia nie dotyczą środków wypłacanych przez państwowy fundusz celowy, jakim jest Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Przedmiotowy projekt ma na celu wprowadzenie zmian, które skutkować będą jak najbardziej efektywnym wykorzystaniem środków funduszu.

Rozwiązanie to jest spójne z obowiązującymi zwolnieniami podatkowymi dla beneficjentów programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery, w tym chodzi o zwolnienie z podatku dotacji otrzymywanych w ramach programów „Czyste powietrze” i „Mój prąd” Wsparcie wdrożenia elektromobilności poprzez zwiększenie nakładów finansowanych związanych ze zwolnieniem dopłat z podatku dochodowego przyczyni się do zwiększenia zainteresowania oferowanymi formami wsparcia oraz efektywnego wykorzystania dopłat, co będzie skutkowało redukcją emisji substancji szkodliwych dla środowiska. Wysoka Izbo! Mam nadzieję, że proponowane zmiany uzyskają poparcie wszystkich środowisk politycznych. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Otwieram dyskusję.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Prawo i Sprawiedliwość w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, druk nr 68.

W obecnym stanie prawnym świadczenia te podlegają ogólnym regułom opodatkowania dochodów, a więc stanowią przychód osób czy podmiotów otrzymujących takie świadczenie i nie są zwolnione od podatku dochodowego ani na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projektowana ustawa przewiduje wprowadzenie zwolnienia od podatku dochodowego, zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, finansowanych ze środków funduszu. Rozwiązanie to jest spójne z obowiązującymi zwolnieniami realizowanymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz poprawy jakości powietrza w naszym kraju. Zdaniem projektodawców wprowadzone zwolnienie korzystnie wpłynie na wzrost użytkowania m.in. pojazdów niskoemisyjnych i przyczyni się do upowszechniania i przyspieszenia transformacji rynkowej w kierunku dalszego ograniczania emisji szkodliwych substancji i poprawy jakości powietrza w Polsce. W związku z tym, że projektowana ustawa jest korzystna dla sektora gospodarki finansów publicznych i nie wpływa na budżety jednostek samorządu terytorialnego, klub Prawo i Sprawiedliwość będzie popierał ten projekt ustawy. Dziękuję bardzo. Pani poseł Leszczyna prosiła o przesunięcie swojego wystąpienia, w związku z czym w tej chwili głos zabierze pan poseł Dariusz Wieczorek w imieniu klubu parlamentarnego Lewica. Bardzo proszę. Na pozór wydaje się, że przedstawiany projekt ustawy dotyczy tylko i wyłącznie spraw związanych z podatkami, bo takie są jedyne zdania dopisane do projektu, do ustawy o podatkach. Natomiast prawda jest taka, że dotyka się tu bardzo istotnej kwestii, a mianowicie kwestii rozwoju elektromobilności w Polsce.

Już wtedy wydawało się to mało realne. Niemniej w tym zakresie musimy zrobić wszystko jako polski rząd, polskie władze, ażeby elektromobilność w Polsce rozwijać. Kwestia tego projektu ustawy to jest ostatnia rzecz w tym łańcuchu rozwoju elektromobilności, bo to jest wprost zniesienie podatku od kwot, które będą dotacjami przy zakupie aut elektrycznych. Natomiast żeby doszło do zakupu auta elektrycznego, musimy przejść wiele różnych procesów. Otóż przede wszystkim jeżeli chodzi o kwestie związane z produkcją aut elektrycznych, to dzisiaj trzeba zapytać, na jakim etapie jest projekt polskiego auta elektrycznego, które przecież parę lat temu zapowiadaliśmy, trzeba zapytać, co dzieje się z fabrykami, które miały produkować autobusy elektryczne, które w tej ustawie są tak istotne, mówię o ustawie o elektromobilności, które są tak ważne, jeżeli chodzi o transport publiczny. W tym zakresie oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia. I tu apelujemy o to, ażeby te działania przyspieszyć, bo ustawa o elektromobilności z 2018 r. już została zmieniona - została ona zmieniona w wielu punktach - i daty, które tam były zapisane, zostały przesunięte. A więc to są działania po stronie państwa, po stronie legislacji, po naszej stronie. Natomiast mamy dwa bardzo istotne podmioty, które w tym procesie muszą uczestniczyć, a które dzisiaj w mojej ocenie, w naszej ocenie w żaden sposób nie są w tym zakresie wspierane.

To muszą być działania, które będą wspierane z pieniędzy budżetowych, bo inaczej tego nie zrobimy. Dzisiaj samorząd przede wszystkim musi się zająć szkołą, chodnikiem, rurociągiem, a dopiero ostatnią pozycją jest rozwój stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie danej gminy, czy też zakup tychże samochodów, bo przecież ustawa o elektromobilności, nawet ta zmieniona, nakłada obowiązek zakupu 10% taboru w samorządach jako taboru, który będzie elektryczny. Drugą grupą, która jest bardzo istotna w tym wszystkim, są firmy energetyczne. I tutaj w tym zakresie jest bardzo wiele do zrobienia. Dzisiaj mamy wrażenie, że jeżeli chodzi o kwestie związane z elektromobilnością, to w przypadku koncernów energetycznych jest to sprawa, która stanowi po prostu tylko i wyłącznie obciążenie. Nikt się de facto tym nie zajmuje, nikt nie przygotowuje infrastruktury, a przecież do stacji ładowania potrzeba infrastruktury energetycznej. W tym zakresie potrzeba również rozwiązań ustawowych, potrzeba decyzji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, potrzeba uwzględnienia tych wszystkich kosztów w taryfach firmy energetycznej, bo bez środków finansowych nie da rady wybudować stacji ładowania samochodów.

Będziemy popierali skierowanie tego projektu do prac w komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Klub Parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 również dołącza się do tych, którzy widzą sens w procedowanym projekcie ustawy. Faktycznie mamy wielki problem przede wszystkim ze stanem powietrza, zwłaszcza w większych ośrodkach, wynikający z rosnącego natężenia ruchu pojazdów, tych pojazdów, które emitują niestety niezmiennie ciągle wiele zanieczyszczeń. Mimo ambitnych zamierzeń, planów ciągle pojazdów elektrycznych nie widać na ulicach polskich miast.

Wydaje się, że to rozwiązanie, które zostało zaprezentowane w przedstawionym projekcie ustawy, wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, przede wszystkim, tak jak powiedziałem, oczekiwaniom Polaków, którzy widzą taką potrzebę.

A więc, tak jak zaznaczyłem na wstępie, nasz klub jest za tym, aby przyjąć zaproponowane w projekcie ustawy zmiany. Dziękuję bardzo, panie pośle.